Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Marcina Duszka, Daniela Milewskiego, Martę Kubiak i Agatę Borowiec. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Marcin Duszek i Daniel Milewski. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Marcin Duszek i Marta Kubiak. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 9, - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9,

W dniu dzisiejszym odbędą się również posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych - godz. 10, - Parlamentarnego Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej - godz. 11, - Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Międzynarodowej Wymiany Kulturalnej - godz. 12, - Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej - godz. 16, - Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej - godz. 17. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o rządowych projektach ustaw: - o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r., - o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2766 i 2767. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, druk nr 2763. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2731)

Panie Marszałku! W imieniu wnioskodawców.

Głównym założeniem tej ustawy było przywrócenie rozwiązania, według którego minister sprawiedliwości sprawował urząd prokuratora generalnego.

Sygnalizowaliśmy wówczas niebezpieczeństwa, które będą się wiązały z rozdzieleniem funkcji urzędu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, i jednocześnie zapowiedzieliśmy, że w momencie kiedy wygramy wybory, to rozwiązanie zostanie przywrócone.

Jeżeli nie zgadzamy się z określonym rozwiązaniem, proponowanym przez większość rządzącą.

Chodzi także o doprecyzowanie regulacji związanej z wykonywaniem przez prokuratury regionalne obsługi finansowej i administracyjnej wydziałów zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz rozszerzenie legitymacji procesowej prokuratorów pełniących obowiązki służbowe w wydziałach do spraw wojskowych prokuratur okręgowych oraz w działach do spraw wojskowych prokuratur rejonowych do występowania przed wojskowymi sądami garnizonowymi oraz przed wojskowymi sądami okręgowymi. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz w oddziałowych komisjach ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, a także o dokonaniu zmian terminologicznych i językowych w treści art. 93 Prawa o prokuraturze oraz o stworzeniu regulacji dotyczących rozszerzenia możliwości delegowania prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Prawa o prokuraturze możliwości określenia w rozporządzeniu wydanym na tej podstawie przypadków, w których nie przysługują diety, o których mowa w art. 109 § 1 Prawa o prokuraturze.

Prawo o prokuraturze poprzez jednoczesne wskazanie, iż wymogi dotyczące osoby ubiegającej się o mianowanie na stanowisko asesora prokuratury spełnia również osoba, która była zatrudniona przez co najmniej 3 lata na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego. Te propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska prokuratorów, ale również wynikają z analizy działania obecnej ustawy. Jeżeli chodzi o zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych zawarte w nowelizacji tejże ustawy, to proponuje się szereg zmian o różnym stopniu istotności i szczegółowości nakierowanych na usprawnienie funkcjonowania sądownictwa powszechnego. Również w tym wypadku ta propozycja stanowi efekt analizy stosowania obecnie obowiązujących rozwiązań, także wprowadzonych w ostatnim czasie, i służy ich korekcie w taki sposób, by można było wyeliminować utrudnienia w sprawnym prowadzeniu postępowań sądowych oraz zapewnić jeszcze skuteczniejsze otoczenie administracyjnego funkcjonowania sądownictwa powszechnego.

umożliwienie prezesowi sądu rejonowego powoływanie przewodniczących wydziałów w kierowanym przez niego sądzie - co obecnie należy do kompetencji prezesa, przełożonego sądu okręgowego - w celu urealnienia nadzoru nad podległym sądem sprawowanego.

Zmiany art. 12 i 16 prowadzą do umożliwienia bardziej elastycznego zarządzania sądami poprzez odstąpienie od zasady, w myśl której każdy sąd rejonowy i okręgowy musi dzielić się na wydział cywilny i karny. Pozwoli to na tworzenie dla tych samych obszarów sądów jednorodnych, wyspecjalizowanych w ramach określonej gałęzi prawa.

Ponadto zmieniono też zasady udziału w konkursie określone w art. 57 i 57aa, które przewidują zarówno możliwość jednoczesnego udziału w dwóch postępowaniach w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym - dotychczas było to możliwe wyłącznie w zakresie jednego konkursu - jak i umożliwiają skuteczną rezygnację z ubiegania się o wolne stanowisko już wskutek złożenia oświadczenia woli w tym przedmiocie. Jeżeli chodzi o zmiany w krajowej szkole sądownictwa, to jest to długo oczekiwana propozycja wprowadzenia aplikacji uzupełniającej.

Nabór na aplikację sędziowską będzie odbywał się w drodze konkursu, zaś na aplikację prokuratorską - w drodze skierowania przez prokuratora krajowego. Aplikacja będzie trwała 18 miesięcy, a zatem o połowę krócej od dotychczasowych, zaś zajęcia będą realizowane w weekendy, tak by nie uniemożliwić aplikantom świadczenia pracy.

Zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego Sądu Najwyższego.

Zmiany art. 34 z kolei gwarantują wyłączenie możliwości obstrukcji postępowań nominacyjnych poprzez wprowadzenie normy wskazującej, że odwołanie od uchwały obejmującej rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego nie wyłącza uprawomocnienia się jej w zakresie, w jakim rozstrzyga o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a jedynie w przypadku jej uwzględnienia daje kandydatowi możliwość uwzględnienia jego wniosku w najbliższym niezakończonym postępowaniu nominacyjnym. Zmiany te umożliwiają także już na etapie kontroli dokonywanej przez Krajową Radę Sądownictwa odrzucenie tych odwołań, które złożone zostały po terminie i nie spełniają wymogów formalnych lub z innych przyczyn pozostają niedopuszczalne. Jeżeli chodzi z kolei o zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, to gwarantują kandydatowi do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego możliwość złożenia dodatkowych dokumentów w postępowaniu nominacyjnym w celu wskazania posiadanych kwalifikacji do objęcia tego stanowiska, jednocześnie zaś wprowadzają rygor pozostawienia bez rozpoznania tych zgłoszeń, które nie spełniają wymogów lub zostały dokonane przez osoby niespełniające jednoznacznych formalnych kryteriów do objęcia stanowiska albo zostały złożone po terminie, w celu jednoznacznego uregulowania sposobu postępowania w takich przypadkach. Natomiast nowe brzmienie art. 111 § 5 służy umożliwieniu szybszego, z pożytkiem dla funkcjonowania Sądu Najwyższego, doprowadzenia do powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego już po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Nienależnie od powyższego w ustawie o Sądzie Najwyższym wprowadzono opisaną już wcześniej zmianę przewidującą utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie dopuszczalności ubiegania się jednocześnie wyłącznie o jedno stanowisko w tym sądzie. Brak zmiany art. 31 § 2 tej ustawy wobec odesłania w zakresie nieuregulowanym ustawą o Sądzie Najwyższym do ustawy o ustroju sadów powszechnych mógłby dawać podstawy do twierdzenia, iż także w Sądzie Najwyższym można ubiegać się jednocześnie o więcej niż jedno wolne stanowisko. Z kolei zmiany dotyczące art. 117 ustawy o Sądzie Najwyższym służą złagodzeniu skutków wejścia w życie przepisów nakazujących sędziom posiadającym także obywatelstwo państwa obcego zrzeczenie się obywatelstwa pod rygorem wygaśnięcia stosunku służbowego, dają bowiem sędziemu możliwość zachowania zajmowanego stanowiska sędziowskiego bez zrzekania się obywatelstwa polskiego. Przepisy przejściowe ustawy gwarantują z kolei możliwość stosowania nowych, usprawniających procedurę nominacyjną regulacji wprowadzonych ustawą także do postępowań o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie. Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne. natomiast skutki finansowe zostaną pokryte w ramach odpowiednich limitów w częściach budżetowych. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem europejskim.

Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Głos ma pan poseł Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec ustawy o zmianie Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli wyzbędziemy się argumentów natury politycznej, to tę ustawę należy określić jako ustawę techniczną, która porządkuje wiele materii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Ustawa o prokuraturze została wprowadzona w życie ponad 2 lata temu i już dzisiaj analiza jej obowiązywania, jej funkcjonowania, jej aspekty, wskazują na to, że jest wiele punktów, wiele miejsc, które wymagają poprawy, doprecyzowania. Jak państwo przeczytają te artykuły, jak państwo poświęcą trochę czasu na to, to okaże się, że rzeczywiście. były problemy praktyczne w wielu miejscach, były pewne miejsca, które całkowicie. Panie marszałku, jeśli można zdyscyplinować przedstawicieli opozycji, to bardzo proszę.

Dzisiaj się okazało, że prokuratura pracuje efektywniej.

Jeśli chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych, jeśli chodzi o ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, to dokładnie w tym samym kierunku zmierzają zmiany. Wielokrotnie przedstawiali państwo uwagi o nieobsadzonych wakatach, wielokrotnie państwo wskazywali również na okoliczność, że. tym oczekiwaniom. Jest uproszczona procedura dochodzenia do zawodu sędziego, jest aplikacja uzupełniająca. To wszystko powinno spowodować, że te braki kadrowe w sądzie będą. rzeczywiście uzupełniane. Mówili państwo o nieefektywności działania Krajowej Rady Sądownictwa. My proponujemy rozwiązania, które. Krajowa Rada Sądownictwa będzie stosowała uproszczoną procedurę weryfikacji kandydatów na sędziów, weryfikacji dokumentów, które przedstawia się w trybie konkursowym, przy powoływaniu sędziów. Oczywiście przedmiotem wielkiego zainteresowania jest ta część, która dotyczy Sądu Najwyższego. ale jeżeli przyjrzymy się dyskusji toczonej przy wprowadzaniu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, to okazuje się, że państwo.

Zatem te uwagi, które były składane wcześniej, ale też praktyka stosowania ustawy od 3 kwietnia, pokazują, że te zmiany są konieczne. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał te zmiany.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wysoki Sądzie, bo warto wam przypomnieć jedną rzecz, słuchajcie, a mianowicie to, że państwo bez wolnych sądów to tak naprawdę jest koniec demokracji, to jest wyprowadzenie nas na kompletny margines cywilizacji europejskiej. Ale co ważniejsze, państwo bez wolnych sądów to jest państwo, które sprzyja cwaniakom, to jest państwo [[Oklaski]] chronienia układu, waszego układu. Kończycie zamach w tej chwili na polskie sądownictwo. I oczywiście pytanie się nasuwa nam wszystkim: Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego tak długo? Bo nie spodziewaliście się takiego oporu na ulicach, [[Oklaski]] , bo nie spodziewaliście się, że polscy sędziowie nie będą się chcieli wam podporządkować. Sposób przygotowania zmian pokazuje, jacy jesteście skrajnie nieprofesjonalni. Kolejne nowelizacje, tak jak to było z Trybunałem Konstytucyjnym, tydzień po tygodniu. Ale wiecie, co to pokazuje? To, że tu nie chodzi o żadną przygotowaną reformę - żadną przygotowaną reformę - tu chodzi tylko i wyłącznie o plan przejęcia sądów. Chcecie wysłać do Sądu Najwyższego kompletnych dyletantów, tak jak to zrobiliście w KRS-ie, tak jak to zrobiliście w Trybunale Konstytucyjnym. No i oczywiście my pytamy, wszyscy posłowie opozycji, ludzie na ulicach pytają: Dlaczego wy to robicie, po co? Żeby bronić swoich interesów. Taka jest odpowiedź. Żeby bronić nowej nomenklatury, którą chcecie stworzyć, i dyktatury ciemniaków. Taka jest odpowiedź. Ja pytam, jakie są elementy waszej reformy, które tak naprawdę poprawią życie zwykłych Polaków. Rządzicie już 3 lata. Niedługo może my będziemy mogli wreszcie skandować. 3 lata, i pytanie jest takie, czy prokuratura, tak jak to było powiedziane przed chwilą, rzeczywiście działa w sposób bardziej efektywny. No to są wolne żarty. Czy sądy działają szybciej? A przypominam, że 3 lata rządzicie. Nie działają szybciej, dlatego że w tej waszej niby-reformie wcale nie chodzi o to, żeby pomóc zwykłym ludziom. Ostatnio okazało się, po co przejęliście Trybunał Konstytucyjny. Po co przejęli Trybunał Konstytucyjny? Ano po to, żeby zapewnić nietykalność swoim kumplom. O to po prostu chodziło [[Oklaski]] - to jest takie proste - żeby prezydent mógł zapewnić nietykalność waszym kumplom, nawet zanim zostaną skazani prawomocnym wyrokiem. Glejty o nietykalności będą sobie wydawać. Tak to będzie wyglądało. Chcecie zwalczać układy? No przecież to są wolne żarty. Swój własny układ chcecie w ten sposób wzmacniać. Podobno rządzący chcą wyjaśnić aferę Amber Gold. No były złośliwości względem pana ministra, i tyle, jakieś dziwne oświadczenia. A pytanie od nas, ale również od ludzi na ulicach jest bardzo proste: Kiedy wy wreszcie zaczniecie wyjaśniać swoje afery? Nigdy. Jak zdeformujecie sądy, wydacie sobie glejt na nietykalność. Ale wiecie, co pokazuje waszą największą słabość? Największą słabość pokazuje to, co się dzieje na ulicach.

To pokazuje waszą słabość, dlatego że się po prostu boicie ludzi, odgradzacie się od nich. Dokładnie tak samo jak mój konkurent - nie wiem, czy wiecie - na spotkaniach w Warszawie. Tam jest bramka, tam się wpuszcza tylko tych ludzi, którzy będą klaskać i będą zadawać właściwe pytania. No tak to wygląda po prostu. Tak to wygląda. Mamy do czynienia, panowie ministrowie, z kolejnym totalnym bublem pary: Ziobro, Jaki. Bo wyście nie potrafili przygotować jednego planu. Wtedy można by było wierzyć w to, że mieliście jakiś plan zmiany sądów. Tylko wy musicie cały czas poprawiać. Nie umiecie niczego nawet przewidzieć, tacy jesteście profesjonalni, fantastyczni. Ciekawe, ile razy i jak wiele rzeczy będziemy musieli po was poprawiać - mam nadzieję, że jak najszybciej. Najpierw pan minister Jaki - pamiętacie, jak występował we wszystkich programach telewizyjnych, codziennie był w telewizji - mówił, jaką fantastyczną przygotował ustawę, a jak się okazało, że to jest idiotyzm 20-lecia, to co się stało? To powiedział jak zwykle, bo oni tylko to potrafią: wina Tuska, i się ulotnił. Pamiętam, jak tam z tyłu nie było go widać. To tak dokładnie będzie wyglądało. Tylko pamiętajcie o jednym - słuchajcie - rozliczymy was z tego. I to mówię też do tych wszystkich ludzi, którzy tu byli na ulicach i którzy dalej na tych ulicach są. Sekundę, sekundę. Panie pośle Trzaskowski, wszystko rozumiem, tylko miałbym prośbę, żeby pan nie obrażał Straży Marszałkowskiej, dobrze? Bo to jest po prostu nieeleganckie. Bardzo proszę, pan poseł Borys Budka, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Ale to jest dowód na to, że nigdy nie było żadnej reformy. Od samego początku chodziło wam o kadry. Zrobiliście to z premedytacją. Zablokowaliście najpierw Trybunał Konstytucyjny, wysyłając tam osoby, które udają sędziów, udają prezesa, tylko po to, by wasza nomenklatura była nietykalna. Krajowa Rada Sądownictwa tak naprawdę stała się przybudówką Nowogrodzkiej. To, co pokazała KRS, udowadnia, że nie ma żadnej reformy. Jeżeli prokurator stanu wojennego rozlicza sędziego Zabłockiego, to to pokazuje wasz stan umysłu. Jesteście największymi hipokrytami w dziejach III RP. Co więcej, już nawet nie kryjecie, że chodzi tylko o to, by szybką ścieżką, poprzez partyjną Krajową Radę Sądownictwa, do Sądu Najwyższego wpuścić takich Misiewiczów wymiaru sprawiedliwości. Przewidujecie, że bez żadnego trybu - to, co wasz szef najbardziej lubi - możecie umieścić w Sądzie Najwyższym klasyczne BMW - biernych, miernych, ale wiernych. Chcecie wsadzić do Sądu Najwyższego sędziów o zerowych standardach moralnych, sędziów, którzy będą ulegli tej władzy. Dlaczego? Właśnie dlatego, by uniewinniać tych, którzy będą, tak jak w tej chwili, doić Polskę na wieleset milionów złotych. Bo przypomnę, Trybunał Konstytucyjny stwierdził. że politycy PiS mogą być nietykalni, jeśli tylko własny prezydent wyda odpowiedni glejt. Nie ma żadnej reformy Sądu Najwyższego, nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Procesy w sądach trwają dłużej, bo minister Zbigniew Ziobro zablokował już w tej chwili blisko tysiąc etatów sędziowskich. Dlaczego to zrobił? Otóż czekał na to, by partyjna Krajowa Rada Sądownictwa była w stanie na te miejsca wpuścić prokuratorów, wpuścić prawników na usługach waszej partii, opłacanych przez spółki Skarbu Państwa, żeby później wydawali odpowiednie wyroki. A Sąd Najwyższy ma wam służyć do trzech celów. Po pierwsze, nowy pseudoprezes Sądu Najwyższego będzie szefem Trybunału Stanu. Ale obiecuję, was ten Trybunał Stanu nie ominie. Nie jesteście w stanie się schować za nowym prezesem Sądu Najwyższego. Druga rzecz bardzo istotna. Zmieniacie ordynację wyborczą tylko dlatego, żeby pozbyć się mniejszych ugrupowań, bo wiecie doskonale, że przegracie te wybory. Współczuję naszym kolegom z tej strony, że dali się wam omamić, bo teraz dopiero widać, co chcecie z nimi zrobić. Ale za pomocą Sądu Najwyższego chcecie wprowadzić scenariusz awaryjny. Przegracie najbliższe wybory samorządowe i będziecie próbowali przez Sąd Najwyższy wpuścić do polskich miast i miasteczek PiS-owskich komisarzy z nadania pana premiera Morawieckiego. Ale obiecujemy: To wam się nie uda. I wreszcie trzecia, bardzo istotna rzecz. Chcecie wyrzucać z sądów, chcecie pozbawiać uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego czy adwokata tych wszystkich, którzy stoją po stronie obywateli, dlatego że wy genetycznie nienawidzicie niezależności, wy genetycznie boicie się niezawisłości, wy tkwicie cały czas w ustroju PRL-u, gdzie była jednolitość władzy państwowej. I dokładnie to w tej chwili wprowadzacie. Przejęliście Trybunał Konstytucyjny, upartyjniliście Krajową Radę Sądownictwa, a teraz Sąd Najwyższy ma być na pasku Nowogrodzkiej. Kochani, nie dajcie sobie wmówić, że jest jakakolwiek reforma.

Bardzo proszę, pan poseł Paweł Grabowski, Kukiz’15. Wysoka Izbo!

Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, ale tak naprawdę to powinno się nazywać projektem ustawy albo projektem projektu ustawy, wersją roboczą projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Drodzy państwo, jeżeli mieliście okazję czytać uzasadnienie tego projektu. Tak żałosnego poziomu już dawno nie widziałem. Literówka na literówce. Drodzy państwo, informuję, że wiem, że korzystaliście z edytora tekstu. W edytorze tekstu jest opcja autokorekty. Przepuszczajcie swoje projekty ustaw przez autokorektę, [[Oklaski]] bo to naprawdę śmiesznie wygląda, kiedy brakuje liter w wyrazach. To po pierwsze. Państwo dużo krzyczycie, korzystacie ze swoich mediów, mediów wam przychylnych, i zakłamujecie rzeczywistość. Tak jest. Proszę się uspokoić, pani poseł, jakieś leki zażyć. Głosowanie nr 89 na 46. posiedzeniu Sejmu. w dniu 20 lipca 2017 r., czyli pierwsza reforma, pierwsza próba reformy Sądu Najwyższego, z zeszłego roku, niebawem będzie rocznica. Gdzie Kukiz popierał tę reformę? Później był projekt prezydencki. Zobaczymy, czy za chwilę odpowiecie.

Pan mówi, że tłumaczą się winni i słabi, a ja mówię, że twardziele pokrzykują nieustannie, jak na bazarze, z sali. Tak się pan zachowuje.

Platforma głosowała razem z PiS-em. To sobie zobacz, człowieku, wyniki głosowań, jak głosowałeś.

Głosowaliście razem z PiS-em za skróceniem kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Drodzy Państwo! Odsyłam wszystkich do głosowania nr 123. Zobaczcie sobie. PiS zagłosował za. Tak wygląda prawda, drodzy państwo. Platforma głosuje razem z PiS-em, a później przeciwko temu wyciąga ludzi na ulice. Brawo! Jesteście w stanie państwo wyjaśnić, jak to jest, drogie kierownictwo? Czemu teraz nie krzyczycie? Czemu teraz nie krzyczycie? Dobra, idziemy dalej. Zgoda. A sędzia na telefon to za czyich czasów był? Jak to się stało, że 7 czy 8 lat waszych rządów skończyło się dziesiątkami postępowań prokuratorskich, CBA itd. Bo wy macie taki styl polityki bazarowej. Panie pośle, sekundę. Zaraz będziecie mnie prosić, żebym dał więcej czasu na pytania. Jeżeli będziecie się tak zachowywać, to nie dam więcej czasu. pan Nitras pokrzykuje, pan Kierwiński jakiś nabuzowany. Wyluzujcie, spokojnie. Idziemy dalej, drodzy państwo. Trybunał Konstytucyjny.

Po co? Po to, by później nikt nie podważał wyroków tego trybunału. Nie jesteście za tym, żeby trybunał stał ponad tym wszystkim, bo nie poparliście tego projektu, niestety. Czy wam się w głowach coś nie pomieszało czasem? Tylko Trybunał Konstytucyjny jest władny orzekać o tym, czy dany projekt jest zgodny z konstytucją, czy nie, a co więcej, drodzy państwo, przypominam. Uspokójcie się, nie zakrzyczycie mnie. Art. 7 konstytucji wprowadza zasadę legalizmu, która stanowi, że wszyscy są zobowiązani działać w ramach i w granicach prawa. obecnie obowiązującego. Idziemy dalej, drodzy państwo. Projekt zawiera wiele propozycji organizacyjnych, sanujących itd., itd.

Wiele spraw można było ogarnąć, załatwić wcześniej, np. kwestię przerywania okresów zasiłkowych urlopami. Przecież to jest stara praktyka. Mało tego, piszecie w uzasadnieniu, że nowelizacja art. 110 ustawy o sądach powszechnych jest konieczna z uwagi na pominięcie w noweli z dnia 8 grudnia 2017 r. jakiejś tam kwestii. To wy sami się przyznajecie, że pominęliście pewne kwestie przy nowelizacji? No to uczciwi, ale to jest nieprofesjonalne, panie pośle. Racjonalny ustawodawca działa na takiej zasadzie, że przedstawia propozycję, poddaje ją pod konsultacje i w wyniku tych konsultacji osiąga konsensus. Wy nie chcecie żadnego konsensusu.

Oto, co się wczoraj działo: przyjeżdżam do Sejmu i strażnik marszałkowski pyta się mnie, czy mam czysty bagażnik, czy nie przewożę ludzi w bagażniku.

To wszystko jest efektem tej konstytucji, którą mamy, że posłowie są odpowiedzialni przed swoimi szefami i kto się mocniej buja na linie, kto jest bardziej miły dla szefa, ten jest tutaj w Sejmie. bo w bagażniku rowerowym nie można nikogo przemycić. Cytuję: Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne. Jakie są pozytywne skutki społeczne? Drodzy państwo, sytuacja społeczna wygląda tak: Sejm stał się zamkniętą i oblężoną twierdzą, co jakiś czas przed Sejmem pojawiają się zasieki, po to żeby wzniecić emocje, stworzyć wrażenie, że tu, nie wiem, będzie wojna. Do tego zmierzacie, drodzy państwo. jest zmiana ordynacji do Parlamentu Europejskiego, która jest wstępem do zmiany ordynacji do Sejmu.

Natomiast problemem jest to, że w przypadku ordynacji do Sejmu, jeżeli będziecie chcieli zmienić ordynację, a wszystko na to wskazuje, że będziecie chcieli stworzyć PO-PiS w polskim parlamencie, tak naprawdę cofniemy się do czasów głębokiego PRL-u, gdzie władza była w rękach pewnej jednej grupy. tylko że dzisiaj ta grupa jest podzielona na Prawo i Sprawiedliwość i PO, czyli razem jest koalicja PO-PiS-u.

Wysoka Izbo! Pan poseł Grabowski jest jednym z niewielu posłów, któremu ABW nie udzieliło dostępu do informacji, certyfikatu o dostępie do informacji niejawnych ABW, więc nawet PiS i jego państwo nie obdarza pana zaufaniem. A więc ja mam pytanie: Kto panu pisał to przemówienie? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po prostu się boicie, najzwyczajniej w świecie się boicie, bo już niedługo tej ustawie o czystkach w Sądzie Najwyższym, tej ustawie będzie mógł się przyjrzeć Trybunał Sprawiedliwości. Stąd ta panika, stąd to ekspresowe tempo prac nad tą ustawą o politycznych dożynkach nad polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeśli mówicie, że przeprowadzacie tą ustawą reformę sądów, to jest tak jakby jakiś bandyta, bijąc po twarzy brutalnie kastetem, mówił, że przeprowadza operację plastyczną. Nigdy nie lubiliście sytuacji, w której ktokolwiek niezależny patrzy wam na ręce. Dlatego najpierw sparaliżowaliście Trybunał Konstytucyjny, potem zajęliście się KRS-em, a w międzyczasie próbowaliście wyrzucić dziennikarzy z Sejmu. Dlatego dzisiaj chcecie po prostu uciec przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Boicie się orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, więc spieszycie się, chcecie działać metodą faktów dokonanych. PiS boi się nawet przyznać, o czym jest ta ustawa, którą dzisiaj rozpatrujemy. I choć dotyczy tak naprawdę drastycznego zwiększania kontroli nad sądownictwem przez polityków PiS-u, to nazwano ją ustawą o prokuraturze. Ta ustawa otwiera bardzo szeroko wrota do tego, aby w sposób bezprawny i błyskawiczny powołać dublera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Podwójna obsada stanowisk, czyli prawna patologia, staje się w państwie PiS standardem, normą. Trzech dublerów sędziów mamy już w Trybunale Konstytucyjnym. Dublerzy członków zostali właśnie skierowani do Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz za pomocą tej ustawy PiS chce w ekspresowym tempie ubiec Trybunał Sprawiedliwości i obstawić, obsadzić stołek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To właśnie dzięki tej ustawie wybór dublera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie możliwy, gdy w Sądzie Najwyższym będzie obsadzonych zaledwie 2/3 etatów. Trzeba powiedzieć głośno, jak na mocy tej ustawy wygląda w skrócie droga do zostania sędzią Sądu Najwyższego w państwie PiS: wymagań merytorycznych wobec kandydata - brak, potrzeby przedstawienia dokumentów - brak, drogi odwoławczej od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa - brak. Czy w takim razie wszystko, czego będzie trzeba, to będzie sympatia polityków z Nowogrodzkiej? To jest jedyne wymaganie? Czy ten konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym jest tak naprawdę już w tym momencie ustawiony? Czy na biurku prezesa PiS leży już w tym momencie lista zwycięzców tego konkursu? Czy ten cały konkurs to przypadkiem nie jest szopka? Przecież wy już pewnie wiecie, kto wygra ten konkurs. Lista patologii prawnych, które są wprowadzane tą ustawą, jest niezwykle długa, tak jak np. wspomniany brak odwołań od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. W skrócie: od upolitycznionej decyzji Krajowej Rady Sądownictwa realnie żadne odwołanie nie będzie przysługiwało. Dlaczego? No przecież to jest kpina. To jak jakbyście zaproponowali: żeby zaskarżyć do Sądu Najwyższego prawidłowość przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, to musiałyby je zaskarżyć wszystkie ugrupowania łącznie ze zwycięskim. Czy wyście przyjechali nocnym pociągiem z Moskwy? Ta ustawa doprowadzi do sytuacji, w której jeden polityk PiS-u kontrolujący Policję stwierdzi, że kogoś trzeba będzie ścigać, a potem kolejny polityk PiS-u, który kontroluje prokuraturę, pośrednio sądy, będzie decydował o tym, kogo oskarżyć i kogo skazać. Tak właśnie będzie się działo, ponieważ każda instytucja wymiaru sprawiedliwości będzie podporządkowana politykom PiS-u. I, szanowni państwo, jest jeszcze jedna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę. Wszystkie sznurki do ręcznego sterowania sądami zbiegają się w rękach Zbigniewa Ziobry. Ja nie wiem, gdzie jest pan Jarosław Kaczyński. Od dawna nikt go już nigdzie nie widział. Ale jednego możemy być pewni: że Zbigniew Ziobro już teraz w myślach przymierza jego prezesowskie buty. Szanowni posłanki i posłowie PiS-u, zastanówcie się chwilę. Każda władza, jaką jemu powierzacie, to jest władza także nad każdym z was, nad każdym politykiem PiS-u. I chyba naprawdę nie jesteście na tyle naiwni, żeby uwierzyć w to, że on to wykorzysta wyłącznie do ścigania przestępców. Stare powiedzenie mówi: wrogów ma się we własnej partii, ale w innych partiach to się ma rywali. Niektórzy z was będą jeszcze płakali wskutek tych reform. Kręcicie bat na własną skórę. Politycy dojnej zmiany. nie damy wam na żadnym etapie zapomnieć o tym, że nie macie prawa łamać polskiej konstytucji, łamać polskiej praworządności.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak czyta się ten projekt, nie ma się wątpliwości, że albo przyspieszenie zmian kadrowych w Sądzie Najwyższym, albo wprowadzenie mechanizmów wpływania na sędziów. Jak? Bardzo proszę. Decyzją prezesa sędzia może być przeniesiony z jednego wydziału do drugiego. Do dzisiaj odwołanie przysługiwało do kolegium sądu apelacyjnego, według tego projektu - do Krajowej Rady Sądownictwa. Przy czym, proszę państwa, odmowa, czyli uwzględnienie stanowiska sędziego, nie będzie uzasadniona i nie będzie od tego przysługiwało odwołanie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy sędzia po 10 czy 15 latach pracy w wydziale cywilnym zostaje przeniesiony do wydziału karnego. A to oznaczać będzie, że o tej kwestii, proszę państwa, o przeniesieniu z wydziału do wydziału będą decydować politycy i sędziowie wybrani przez polityków. Tak będzie funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Według tego projektu, a w zasadzie wcześniej na sztandar wyniesiono hasło losowego przydzielania spraw. To miał być sposób na reformę wymiaru sprawiedliwości. I co się dzieje w tym projekcie? Czyli wylosujemy sędziego, a potem do pierwszego posiedzenia, na którym mają być strony, możemy zrobić wszystko, czyli zmienić skład. Wprowadzacie państwo rozwiązanie, które dopiero powoduje niepewność całej sytuacji. Wcześniej to było sztandarowe hasło reformy wymiaru sprawiedliwości, a dzisiaj wprowadzacie rozwiązanie, które pozwoli zmienić sędziego ot tak, bo uznacie, że ten, który został wylosowany, nie jest właściwy. Wprowadzacie państwo rozwiązanie, które przewiduje karanie sędziów, zanim zapadnie prawomocne rozstrzygnięcie, i przewidujecie, że jeżeli sędzia zostanie uniewinniony, to zwróci mu się te pieniądze. No ale gdzie zasada domniemania niewinności? Sędzia zostaje ukarany, zanim prawomocnie skończy się postępowanie. Wprowadzacie państwo rozwiązanie, które przewiduje, że sędzia dostanie pozytywną akceptację pracy w Sądzie Najwyższym, ale możliwe będzie zaskarżenie tej uchwały do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezydent dokona zaprzysiężenia na sędziego Sądu Najwyższego, a Naczelny Sąd Administracyjny wyda orzeczenie, w którym uzna naruszenie prawa przy przyjęciu tej uchwały. Jak będzie wyglądała sytuacja? Jak będą wyglądały orzeczenia tego sędziego, co do którego następnie zostanie to uznane przez Naczelny Sąd Administracyjny za niezgodne z prawem? Wprowadzacie państwo zapis, że prokurator będzie mógł uczestniczyć w każdym postępowaniu, jakiekolwiek sobie wymarzy, ale wprowadzacie ogólną regułę, której nie uściślacie, a to oznacza, że nie będzie wiadomo, w jakim charakterze będzie występował. To jest zrobione specjalnie? Taki macie zamiar? Mnóstwo jest takich rozwiązań, które powodują, że niestety ta ustawa nie może się ostać. Zmierzacie państwo do szybkich zmian kadrowych. Dlaczego? Dlatego że chcecie obsadzić izbę, która rozstrzygnie o ważności najbliższych i kolejnych wyborów. I dlatego tak bardzo skupiliście się na pierwszym prezesie Sądu Najwyższego - bo ta kadencja kończy się w 2020 r., a więc po większości wyborów, w kwietniu 2020 r. A pierwszy prezes Sądu Najwyższego przewodniczy Trybunałowi Stanu. Wprowadzacie państwo rozwiązania, zgodnie z którymi na aplikację uzupełniającą w przypadku sądowej trzeba będzie zdać egzamin konkursowy, ale w przypadku prokuratorskiej zadecyduje już o tym prokurator krajowy - arbitralnie, bo nie ma żadnej argumentacji, żadnych reguł, według których [[Dzwonek]] będzie o tym decydował. Ta ustawa nawet nie powinna znaleźć się w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów chciałbym przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Rzekomo, szanowna większości sejmowa, od roku naprawiacie w Polsce sądy. Piąta nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, piąta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, trzecia nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, druga nowelizacja ustawy Prawo o prokuraturze, druga nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Czy przez ten rok Polakom lepiej korzysta się z wymiaru sprawiedliwości? Czy coś zmieniło się w zakresie skrócenia terminów korzystania z sądów? Nie. Przez rok oszukujecie Polaków rzekomą wolą zmiany wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ja bym dzisiaj chciał skorzystać z okazji, szanowni państwo, i poprosić pana posła wnioskodawcę, pana ministra, żebyście stanęli dzisiaj w tym miejscu, w którym ja teraz stoję, spojrzeli Polakom prosto w oczy i wymienili ten rzekomo obfity katalog tych usprawnień, dzięki którym w sądach powinno być lepiej.

Wówczas też władza chciała mieć po prostu władzę nad sądami. Czy nie wstyd wam, że dzisiaj w Europie i w Stanach Zjednoczonych mówi się o Polsce jako kraju, który się pogubił, który nie rozumie podstawowych prawideł ustroju nowoczesnego państwa? Szkoda, szanowni państwo, zawiedzionych oczekiwań Polaków i szkoda opinii Polski w Europie. Z każdą nową ustawą, która ma go poprawiać, on działa coraz gorzej, wolniej i słabiej. I ten projekt również w swej treści dokładnie pokazuje, co jest motorem napędowym Prawa i Sprawiedliwości. To już nie jest chęć podporządkowania tych sądów, ale coś jeszcze, coś więcej: strach, strach i panika, że przejęcie sądownictwa może się nie udać.

Tu już nie chodzi o 44 miejsca, wakaty w Sądzie Najwyższym.

Przypomnę dzisiaj państwu, którzy nas słuchają, że są 44 miejsca w Sądzie Najwyższym, dwa miejsca wakujące w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dziewięć miejsc w wojewódzkich sądach administracyjnych, 76 miejsc w sądach apelacyjnych, 372 wakaty w sądach okręgowych i 98 miejsc w sądach rejonowych. Te wakaty nie powstały za sprawą opozycji, szanowni państwo. Dzisiaj większość sejmowa, te harce, które wspólnie z ministerstwem prowadzicie od ponad roku, niestety z ubolewaniem trzeba powiedzieć, że również przy istotnym udziale pana prezydenta, powodują takie osłabienie wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa w Polsce. To jest degradacja i coraz gorsza zmiana w tym sądownictwie. Pozwolę sobie na chwilę zatrzymać się przy organie, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, którego działanie też zostało objęte przez procedowany projekt.

W sumie to jest kolejna ustawa, która niczego dobrego nie daje Polakom, nie ma żadnej wartości dodanej. Wnioskujemy o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Głos ma pan poseł Jacek Protasiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Wysoki Sejmie!

Otóż chcę wyraźnie z tego miejsca powiedzieć: nie macie prawa do tej reformy. Nie macie prawa do łamania konstytucji, a w szczególności art. 173, który mówi, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Nie macie prawa do skracania kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która w konstytucji określona jest wyraźnie na 6 lat.

O tym, że to nie jest żaden program, tylko chaotyczny skok na sądownictwo w Polsce, świadczy również biegunka legislacyjna.

Mam tu na myśli pana sędziego Zabłockiego.

Przypomnę tylko cytat z wypowiedzi osoby, która przed komisją senacką mówiła: jeśli chodzi o prawo, to ja jeszcze mogę doczytać, i która została przez was uczyniona ławnikiem w tym najważniejszym z sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Trzecim przykładem jest odbieranie prawa do wypowiedzi tu, w tym Sejmie, na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przez prokuratora stanu wojennego rzecznikowi praw obywatelskich. To jest skandal. I wreszcie czwarta rzecz, może najmniej istotna, ale warto dzisiaj o tym wspomnieć, zwłaszcza że bohaterka tego wątku właśnie pojawiła się na sali. Czwartym symbolem tej deformy, tego skoku, tego skandalu, tego, co wyprawiacie z polskim sądownictwem, są obelgi miotane przez panią poseł Pawłowicz tu, na tej sali, na posiedzeniach komisji i wreszcie w Internecie. Otóż, pani poseł, wczoraj miała pani czelność nazwać lewą część tego Sejmu bydlęciem, bydłem. Otóż chcę pani powiedzieć jedną rzecz. Zasiadam w lewej części tego Sejmu.

I choć domyślam się, że chodzi pani o sprowokowanie porównania tej części sali, pani i pani sąsiadów, do innego oborowego przykładu, to powiem pani, że jednak skorzystam z rady Marka Twaina, który wypowiedział kilkadziesiąt lat temu słowa: nigdy nie dyskutuj z prostakiem, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Panie Marszałku! Ja też siedzę po lewej stronie i solidaryzuję się z moim przedmówcą. Pan Waldemar Buda, poseł sprawozdawca z PiS-u, powiedział coś takiego: jeśli wyzbędziemy się argumentów politycznych, to zobaczymy, że tak naprawdę ta ustawa jest taką zamianą techniczną. Projekt tej ustawy nie jest odpowiedzią na problemy wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego, lecz jest odpowiedzią na aktualną sytuację polityczną związaną z wprowadzeniem przez PiS, czyli przez was, ustaw o sądownictwie. To jest tylko i wyłącznie po to. To nie jest odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości i pan o tym bardzo dobrze wie.

To jest tylko i wyłącznie na zlecenie polityczne. To nie jest ani ustawa, ani reforma, to są wszystko atrapy. To, co robicie, nie zasługuje na to, żeby nazywać to jakąkolwiek reformą. Pana Ziobry też nie można nazywać ministrem sprawiedliwości, bo co to za minister sprawiedliwości? I to jest właśnie ten prawdziwy zamach. To jest zamach, który przeprowadziliście i z którego będziecie rozliczeni. Patrząc na opinię rzecznika praw obywatelskich, jasno widać, że ten projekt budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich. Mówi o tym, że ten wasz projekt prowadzi m.in. do możliwości manipulacji przez prezydenta i premiera przy wyłanianiu kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz do znaczącego ograniczenia samorządności w sądach powszechnych, co było już wcześniej tutaj mówione. Ona pokazuje, jak wy działacie. Chcecie przeprowadzić projekt bez konsultacji, bez opinii, bez uzasadnienia, w 24 godziny. Pokazujecie właśnie, procedując w ten sposób, jak traktujecie suwerena. Traktujecie go jak obcego.